Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Marcina Duszka, Daniela Milewskiego, Łukasza Schreibera i Sylwestra Tułajewa. Proszę pana posła sekretarza o odczytanie komunikatów. Wysoka Izbo!

Dziękuję bardzo. Informuję, że prezes Rady Ministrów zawiadomił Sejm o zamiarze przedłożenia prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie, zmian do Załącznika I do Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzonej w Helsinkach 17 marca 1992 r. Posłowie w określonym terminie nie zgłosili zastrzeżeń co do zasadności wybranego przez Radę Ministrów trybu ratyfikacji tego dokumentu. Komisja Spraw Zagranicznych przedłożyła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie tego zawiadomienia od premiera bez zastrzeżeń. Sprawozdanie komisji to druk nr 2125. W związku z tym, na podstawie art. 120 ust. 4 regulaminu Sejmu, informuję o braku zastrzeżeń co do zasadności wybranego przez Radę Ministrów trybu ratyfikacji tego dokumentu. Prezydium Sejmu przedłożyło wnioski: - w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, - w sprawie wyboru nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Są to odpowiednio druki nr 2130 i 2124. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych wniosków. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 2117 i 2118. W związku z tym, po uzyskaniu odpowiedniej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu oraz aby w dyskusjach nad tymi punktami porządku dziennego wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę rozumiał, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Grupa posłów przedłożyła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Jest to druk nr 2131. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę rozumiał, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Z wnioskiem formalnym zgłosił się pan poseł Jerzy Meysztowicz, klub Nowoczesna. Wysoka Izbo! Na podstawie art. 184 regulaminu Sejmu zwracam się do pana marszałka z prośbą o przerwę. Wczoraj naszemu klubowi odmówiono możliwości zadania w dniu dzisiejszym pytania w sprawach bieżących. Jednoznacznie odbieramy to jako próbę ograniczania praw mniejszości parlamentarnej. Sejm sprawuje nadzór m.in. nad takimi instytucjami jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. To Sejm wybiera jej członków, to Sejm przyjmuje jej sprawozdania. Na tej podstawie zwracam się z prośbą do pana marszałka o wezwanie do Sejmu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pana Witolda Kołodziejskiego, aby wyjaśnił Wysokiej Izbie, jak doszło do nałożenia skandalicznej kary na komercyjną i wolną stację telewizyjną TVN, i to chyba jednej z najwyższych w historii, czyli 1,5 mln zł. Niedopuszczalne jest, że tak tendencyjna i niezgodna z faktami opinia, na którą się powołano, została przygotowana przez osobę związaną z konkurencyjną stacją telewizyjną. Niedopuszczalne jest też, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nakłada karę za materiał, który spełnia wszelkie wymogi rzetelnego dostępu społeczeństwa do informacji. Przypomnijmy, że protest w Sejmie rozpoczął się od poparcia przez posłów opozycji dziennikarzy upominających się o wolne i niezależne media. Demokracja to jest system, który obcy jest obecnie sprawującym władzę.

Jeśli za taką relację zdominowaną przez PiS-owskich nominatów Krajowa Rada

zabrać koncesję.

Otóż klub, którego pan jest członkiem, złożył projekt pytania w sprawach bieżących w tej sprawie, którą pan opisał, ale ze względów formalnych Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii prawników Kancelarii Sejmu uznało, że adresat jest niewłaściwy, ponieważ pytanie zostało zgłoszone do ministra kultury. Jest ona instytucją umocowaną konstytucyjnie, w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym zaproponowałem Prezydium Sejmu. Tutaj sprostowań nie będzie, panie pośle, tak że proszę siadać. W związku z tym zaproponowałem Prezydium Sejmu, żeby zgodnie.

Ale został złożony wniosek formalny, w związku z tym przegłosujemy go. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2100-A. Proszę pana posła Andrzeja Kosztowniaka o przedstawienie tego sprawozdania. Panie Marszałku! Panie Premierze! Szanowni Państwo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych z druku nr 2100-A o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw. W dniu wczorajszym w trakcie drugiego czytania zostały złożone dwie poprawki, które uzyskały pozytywną opinię komisji finansów.

W 1. poprawce wnioskodawcy proponują, aby skreślić ust. 5 w art. 366 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Z tą poprawką łączy się poprawka 2. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2100, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy głosowali za.

Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Piotra Uścińskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Szanowna Rado Ministrów! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. W dniu wczorajszym podczas drugiego czytania została zgłoszona jedna poprawka, aby wydłużyć czas wejścia w życie ustawy do 1 lipca 2018 r. Komisja Finansów Publicznych ze względu na fakt, iż ustawa ma minimalny wpływ na polską gospodarkę i na wpływy budżetowe, natomiast grożące Polsce kary za opóźnienie wejścia w życie postanowień orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są bardzo znaczne, prosi i wnosi o odrzucenie tej poprawki i przyjęcie projektu ustawy bez tej poprawki. Dziękuję panu posłowi. Nad poprawką, o której mowa w dodatkowym sprawozdaniu, głosować będziemy w pierwszej kolejności.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Pytanie zadaje poseł Jerzy Meysztowicz, klub Nowoczesna. Czas na zadanie pytania ustalam na 1 minutę. Wysoka Izbo! Dlaczego państwo nie chcecie się zgodzić, aby przesunąć termin wprowadzenia tej ustawy na 1 lipca 2018 r. Byłaby wtedy możliwość, żeby przedsiębiorcy przystosowali się do nowych warunków, bo zwiększenie akcyzy i dodatkowy podatek dla tych przedsiębiorców jest zmianą reguł prowadzenia działalności gospodarczej.

Niezależnie od wzrostu kosztów utrzymania, wzrostu cen, inflacji, teraz jeszcze wprowadzacie dodatkowy podatek. Czyżby już zabrakło pieniędzy w kasie na wasze obietnice wyborcze? Dziękuję panu posłowi. Oczywiście ten projekt został złożony do Sejmu dość dawno, jeszcze przed zmianą rządu, ale dzisiaj głosujemy nad poprawką. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Do całości projektu ustawy pytanie zadaje poseł Krzysztof Truskolaski, klub Nowoczesna. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niestety pana nie ma, ale przedwczoraj tak pięknie mówił pan o tym, że chcecie obniżać podatki, że chcecie ulżyć Polakom. Pierwsza z nich dotyczyła akcyzy na wyroby tytoniowe, którą obciążyliście małe i średnie przedsiębiorstwa, a teraz podnosicie VAT. Panie premierze, dlaczego po raz kolejny podnosicie podatki? Nowoczesna już niejednokrotnie mówiła, że podatki trzeba obniżać.

Wysoka Izbo!

Obniżyła VAT na książki elektroniczne, bo uważa, że oświata jest ważniejsza niż decyzje takich czy innych biurokratów. Dlaczego my nie mamy tej odwagi? W tej sprawie wypowie się wiceminister finansów pan Paweł Gruza. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Ta ustawa to jest zmiana techniczna, ona ma pomijalne skutki budżetowe. Wymiar finansowy tej ustawy jest nieistotny. Wczoraj miałem przyjemność być w Brukseli. Na forum wszystkich państw dyskutowane są modyfikacje dyrektywy VAT-owskiej w zakresie tego gorsetu, który ogranicza nasze prawo do stosowania stawek obniżonych. Ten proces jest delikatny, on się toczy. W tym momencie ważne jest, żeby technicznie dostosować nasze prawodawstwo do wymogów dyrektywy. Dziękuję. Mamy wyjaśnienie. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem projektu ustawy w całości w brzmieniu z druku nr 2056, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2094. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2094, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy polskiej awangardy. Przystępujemy do głosowania. Komisja wnosi o podjęcie uchwały w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu w druku nr 2077. Kto z pań. Pan poseł?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 2077, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały z druku nr 2076. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 2076, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Jego odrzucenie oznaczać będzie, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego w celu rozpatrzenia. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 1611, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka. Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały z druku nr 2123. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 2123, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 23. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2130) Wysoki Sejmie! Prezydium Sejmu na podstawie art. 20 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Czy ktoś z pań i panów posłów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nikt się nie zgłasza. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 2130, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 24. porządku dziennego: Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2124)

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 2124, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?